Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Piotra Łukasza Babiarza i Sylwestra Tułajewa. Protokół i listę mówców prowadzić będzie pan poseł Piotr Łukasz Babiarz. Wysoka Izbo! Mam wielki zaszczyt powitać dzisiaj podczas naszych obrad przewodniczącego Seimasu Republiki Litewskiej pana Viktorasa Pranckietisa wraz z delegacją. Witamy serdecznie.

Pragnę serdecznie powitać również marszałka Senatu pana Stanisława Karczewskiego. Witam przybyłych wicemarszałków Senatu i państwa senatorów.

Witam wszystkich obecnych. Proszę przewodniczącego Seimasu Republiki Litewskiej pana Viktorasa Pranckietisa o zabranie głosu.

Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli narodu polskiego.

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tu być dzisiaj i występować przed takim dostojnym gremium.

Obchodzimy setne rocznice odzyskania niepodległości przez nasze państwa. W przyszłym roku natomiast obchodzić będziemy inny znaczący jubileusz: 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Jest to więc doskonała okazja do zastanowienia się nad szlakiem pokonanym przez nasze narody, nad naszą wspólną historią i nad tym, co nasz łączy, jednoczy, nad tym, jakie są najważniejsze wyzwania dnia dzisiejszego oraz przyszłości, stojące przed obywatelami Litwy i Polski, co my, politycy, powinniśmy uczynić, aby nasze społeczeństwa miały poczucie bezpieczeństwa, a gospodarki naszych krajów się rozwijały. Jestem przekonany, że właśnie w tym roku jubileuszowym dla naszych krajów prawidłowo wykorzystamy możliwości litewsko-polskiej współpracy parlamentarnej oraz zachęcimy do działania bilateralne zgromadzenie parlamentarne. Pragnę odnotować, że historia nasze narody na przemian łączyła i dzieliła, jednakże przez cały czas więcej w historii było wspólnego niż dzielącego i sprzecznego. Jeszcze od unii w Krewie rozpoczął się niełatwy proces zbliżenia obu państw.

Ta pierwsza konstytucja uchwalona w Europie daje nam doskonałą okazję do refleksji nad znaczeniem i wagą zasad konstytucyjnych. Podczas podróży z Litwy do stolicy Polski, Warszawy, jedzie się przez warszawską Pragę, gdzie na początku listopada 1794 r. podczas powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów przeciwko Rosji ok. 8 tys. żołnierzy Wielkiego Księstwa Litewskiego wraz z żołnierzami polskimi i mieszczanami Warszawy stanęło w obronie Warszawy przed armią rosyjską. W bitwie zginęła większość wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego i obrońców Warszawy. Bitwa ta jest często nazywana rzezią Pragi. Był to ostatni bój z udziałem wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydaje mi się, że podczas obchodów w 2019 r. 225. rocznicy powstania pod wodzą Tadeusza Kościuszki byłoby wskazane upamiętnienie żołnierzy Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy broniąc Warszawy, złożyli w ofierze swe życie. Zniknięcie z mapy Europy Rzeczypospolitej Obojga Narodów rozdartej podczas grabieżczych rozbiorów przez Rosję, Prusy i Austrię w XVIII w. uczy nas dzisiaj, że powinniśmy być silni i gotowi samodzielnie lub wraz ze swoimi sojusznikami przeciwstawić się agresji zewnętrznej sił antydemokratycznych.

Należy ją chronić i pielęgnować, tak jak to czyniła litewska Joanna d’Arc, czyli Emilia Plater.

Drogi Litwy i Polski rozminęły się w okresie międzywojennym z powodu Wilna, jednakowoż oba nasze państwa i narody były niezależne, samodzielnie budowały własną przyszłość, kreowały swój postęp gospodarczy.

Internowano polskich żołnierzy, którzy następnie nie powrócili z Katynia, zaś ich losami cynicznie zarządzali dyktatorzy w Berlinie i w Moskwie. II wojna światowa przyniosła nieobliczalny ból i cierpienie ludzi różnych narodowości, zaś po jej zakończeniu zostaliśmy oddzieleni stalinowską żelazną kurtyną od demokratycznego świata zachodniego. Państwa Europy Zachodniej świętowały zwycięstwo nad nazizmem, natomiast na Litwie, podobnie jak w Polsce, nadal trwał ruch oporu, zwany u nas wojną po wojnie, w którym na Litwie ponad 20 tys. leśnych braci będących uczestnikami podziemnego ruchu oporu oddało swe życie na rzecz naszej dzisiejszej wolności. Zwanych przez system sowiecki wrogami narodu tysiącami deportowano na bezkresy Syberii. Niektórym z nich udało się powrócić do wykrwawionej, okupowanej ojczyzny, wielu z nich jednak pozostało na wieczny spoczynek w miejscach deportacji. Cześć ich pamięci!

Od pierwszych dni swego pontyfikatu często powtarzał on „Nie lękajcie się” Nasze narody to usłyszały, były zatem silne dzięki swej wierze w wolność.

Styczniowe wydarzenia na Litwie przyspieszyły upadek Związku Radzieckiego, który trafnie przez amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana został nazwany imperium zła.

Chciałbym podziękować naszym kolegom z Polski, którzy podczas tych wszystkich wydarzeń byli z nami w Wilnie i pomagali naszym przedstawicielom w innych krajach w dążeniu do zapewnienia wsparcia światowej wspólnoty na rzecz międzynarodowego uznania odzyskania przez Litwę niepodległości.

Szczerze opłakiwaliśmy utratę dobrego przyjaciela Litwy prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

Oczekujemy też w Wilnie na wizytę premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to źródłem inspiracji dla naszej dalszej współpracy.

Stanowimy doskonały przykład udanej transformacji systemowej dla tych krajów, które swą przyszłość wiążą z Unią Europejską, w szczególności dla Ukrainy.

Członkostwo w Unii Europejskiej postrzegamy nie tylko jako dobrobyt gospodarczy i materialny naszych państw i obywateli, ale też jako przynależność do wspólnoty krajów połączonych przez wspólne wartości.

Nielegalna migracja i potoki uchodźców, debata na temat przyszłego modelu Unii Europejskiej, która przyspieszyła wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, populizm i eurosceptycyzm, zapewnienie stabilności finansowej i wzrostu gospodarczego, zmiany klimatyczne, zagrożenia hybrydowe połączone z propagandą, dezinformacją i atakami cybernetycznymi krajów trzecich - to są największe wyzwania i zagrożenia dla Unii Europejskiej, Litwy i Polski.

Mamy nadzieję, że negocjacje w sprawie brexitu będą udane i zachowamy strategicznie ważne partnerstwo oraz zagwarantowane będą prawa naszych obywateli w Zjednoczonym Królestwie. Czekają nas ważne decyzje w sprawie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W nowych wieloletnich ramach finansowych szczególną uwagę należy poświęcić długoterminowym strategicznym zobowiązaniom zawartym w traktatach Unii Europejskiej, znając jednocześnie wartość dodaną polityki spójności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i dobrobytu obywateli.

W biegu dziejów, kiedy Litwa traciła niepodległość, traciła ją również Polska, i odwrotnie.

Jesteśmy również wdzięczni Polsce za aktywne wsparcie naszych wysiłków na rzecz członkostwa w NATO.

Aneksja Krymu przez Rosję oraz wojskowa i polityczna destabilizacja w Donbasie we wschodniej Ukrainie i wspieranie separatystów radykalnie zmieniły sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. NATO to transatlantycki sojusz polityczno-wojskowy, dlatego uwaga polityczna ze strony USA i obecność żołnierzy amerykańskich i innych sojuszników w Polsce i krajach nadbałtyckich są istotnymi czynnikami zapewniającymi skuteczne odstraszanie od potencjalnej agresji, obronę i wzmocnienie sił NATO na całej flance wschodniej. Powinniśmy jednocześnie starać się unikać niepotrzebnego powielania działań NATO i Unii Europejskiej. Należy w pełni wdrożyć unijną deklarację współpracy między NATO a Unią Europejską, uchwaloną podczas szczytu NATO w Warszawie. Aktywna współpraca bilateralna z Polską odbywa się we wszystkich formatach sił wojskowych poprzez ćwiczenia wojskowe, uczestnictwo w operacjach międzynarodowych i zakup broni dla sił zbrojnych. Dziś w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kontrolowane są stare i nieustannie tworzone są nowe wspólne formaty współpracy wojskowej.

Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Polska jest najaktywniejszym krajem w zakresie kontroli przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Już siedem razy Polska delegowała przedstawicieli swych Sił Powietrznych do NATO-wskiej misji obrony przestrzeni powietrznej. Nasze kraje powinny podjąć aktywną współpracę i wymianę doświadczeń w celu wyeliminowania pojawiających się nowych zagrożeń hybrydowych przez zwiększenie odporności naszych społeczeństw na wrogą propagandę i gotowości do reagowania na ataki cybernetyczne. Energetyka to sektor, w którym współpraca naszych krajów jest szczególnie dynamiczna w ostatnich latach.

Jest to pierwsze w historii połączenie energetyczne Litwy z Zachodem. Realizacja projektu synchronizacji systemów energetycznych państw bałtyckich zintegruje państwa bałtyckie z europejskim systemem energetycznym. Wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszych państw, a także dla rozwoju rynku gazu w rejonie będzie miała budowa gazociągu między Polską a Litwą, GIPL. Z zadowoleniem przyjmujemy stanowisko Polski w sprawie elektrowni jądrowej w Ostrowcu na granicy Białorusi z Litwą. W czasie budowy doszło do kilku poważnych incydentów, co wskazuje na to, że obiekt potencjalnie może stanowić zagrożenie dla całego regionu. Litwa żąda, aby podczas budowy tej elektrowni postępowano zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jesienią zeszłego roku parlament litewski uchwalił ustawę zabezpieczającą środki niezbędne do tego, aby na litewski rynek energii elektrycznej nie trafiła energia elektryczna z krajów trzecich, pochodząca z niebezpiecznych elektrowni jądrowych. Mamy nadzieję, że również Polska w przyszłości nie będzie importowała energii elektrycznej z niebezpiecznej elektrowni jądrowej w Ostrowcu.

Widzimy też możliwości rozwijania potencjału w zakresie współpracy krajów Trójmorza w celu dążenia do lepszego rozwoju infrastruktury transportowej i energetycznej państw regionów Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Litwy, a także jednym z najsolidniejszych inwestorów. Z zadowoleniem zauważamy, że coraz więcej litewskich przedsiębiorstw odnosi sukcesy na polskim rynku i konsekwentnie się rozwija. Jestem przekonany, że dzięki wzajemnej życzliwej współpracy otwierają się szerokie możliwości dotyczące poszukiwania trwałych rozwiązań. Spójna polityka gospodarcza Litwy w ostatnich latach stworzyła sprzyjające warunki dla biznesu i atrakcyjny klimat dla inwestycji na Litwie.

Polskim inwestorom oferujemy atrakcyjne warunki inwestowania i szerokie możliwości współpracy. Szanowni Posłowie i Senatorowie!

Naszym celem jest, aby osoby dowolnej narodowości czuły się na Litwie dobrze, będąc przedstawicielami swojego narodu oraz lojalnymi obywatelami swojego kraju. Pragnę odnotować, że Litwa jest jedynym krajem na świecie, rzecz jasna oprócz samej Polski, w którym dla osób polskiego pochodzenia zapewniona jest oświata w języku polskim od przedszkola do szkoły wyższej.

Jest to jedyny polski uniwersytet posiadający swą filię za granicą i kształcący studentów w języku polskim.

Zarówno w Polsce, jak i na Litwie ważna jest dobra znajomość języka urzędowego danego państwa. Młodzież polska na Litwie dobrze zna język litewski, zaś Litwini w Polsce świetnie mówią po polsku. Ważne jest również, aby Polacy na Litwie byli aktywnymi politycznie i społecznie członkami naszego społeczeństwa. W chwili obecnej na Litwie aktywnie działa ok. 70 organizacji, polskich wspólnot narodowych. Zakres ich działalności jest bardzo szeroki: zespoły pieśni i tańca, chóry, stowarzyszenia i kluby, uniwersytet trzeciego wieku. Działają też media w języku polskim.

W Sejmie Republiki Litewskiej interesy polskiej wspólnoty narodowej reprezentuje Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Rodzin Chrześcijańskich posiadająca 8 mandatów z ogólnej liczby 141. Jeden przedstawiciel polskiej narodowości jest posłem w Parlamencie Europejskim. Zwracam się uprzejmie do polskich parlamentarzystów z prośbą o konstruktywne rozstrzyganie kwestii podnoszonych przez społeczność litewską dotyczących szkolnictwa litewskiego, finansowania podręczników i innych kwestii.

Zaplanowane są też w Polsce tygodnie litewskiego kina i teatru, różne wystawy i inne wydarzenia. Chciałbym zaprosić Polaków do odwiedzania multikulturalnej Litwy, gdzie zawsze czekamy na gości z Polski i dobrze ich rozumiemy.

Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej panu Markowi Kuchcińskiemu oraz wszystkim państwu za umożliwienie mi wystąpienia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Patrząc w przeszłość, widzimy też przyszłość. Otwieramy dziś nową kartę w historii Litwy i Polski. Chciałbym również serdecznie wszystkich państwa pozdrowić z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odrodzenia niepodległości Polski.

Niech żyją Polska i Litwa, wolne, demokratyczne i niepodległe kraje rodziny europejskiej!

Dziękuję panu przewodniczącemu Seimasu litewskiego. Zarządzam przerwę do godz. 10.15.

Wznawiam obrady. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - bezpośrednio po zakończeniu głosowań, ok. godz. 11.30, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 11.30, - Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 12, - do Spraw Petycji - godz. 12. Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych: - Parlamentarnego Zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S-12 - bezpośrednio po zakończeniu głosowań, - Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej - godz. 12.30, - Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej - godz. 13. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Wysoki Sejmie! Proszę bardzo. Panie i Panowie Posłowie! W wieku 41 lat zmarł pan Daniel Kozdęba, prezydent Mielca. Był wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Był również absolwentem, a następnie doktorantem Politechniki Rzeszowskiej. Studiował również na Uniwersytecie Warszawskim. Członek komisji przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej, powołany przez premiera Jerzego Buzka, asystent i doradca minister Krystyny Łybackiej, swego czasu wiceprezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dwukrotnie był radnym powiatu mieleckiego, a następnie został wybrany na prezydenta Mielca.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2247-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Wojciecha Zubowskiego o przedstawienie tego dodatkowego sprawozdania komisji. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała jedyną poprawkę do omawianego projektu ustawy i wnioskuje o jej przyjęcie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że chodzi o druk nr 2247. W tej poprawce do art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wnioskodawcy proponują nowe brzmienie dodawanego ust. 3. Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2247, wraz z przyjętą poprawką, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2265-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie tego sprawozdania. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła 22 poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania przedmiotowego projektu ustawy. Komisja rekomenduje również przyjęcie całego projektu ustawy z druku nr 2265. Dziękuję panu posłowi. Przypominam, że chodzi o druk nr 2265. Komisja, przypominam, wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje pani poseł Genowefa Tokarska, PSL - UED. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poprawka dotyczy wykreślenia z projektu zapisu, który mówi, że generalnym inspektorem może być osoba, która wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną. Mam do rządu pytanie, kto, kiedy i w sprawie czego dokona obiektywnej, podkreślam: obiektywnej, oceny tych cech, które tutaj przytaczam. Pragnę zwrócić uwagę, że inne zapisy tego projektu mówią, że inspektorem może być tylko sekretarz lub podsekretarz stanu.

Przecież tutaj pomnażamy to samo, bo w oświadczeniu już musi być to zbadane, stwierdzone.

Pan minister Leszek Skiba, wiceminister finansów, odpowie na pytanie pani poseł. Wysoka Izbo! Pytanie dotyczy patriotyzmu. Wydaje się, że ten zapis już działa w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jest stosowany. Mam wrażenie, że nie będzie w związku z tym żadnych problemów. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Za głosowało 430, nikt nie głosował przeciw, 3 posłów wstrzymało się. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za głosowało 431, przeciw - 1, wstrzymało się 3 posłów. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za głosowało 433, przeciw nikt nie głosował, wstrzymało się 3. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 431, przeciw - nikt, wstrzymało się 3 posłów. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 15. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 16. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 430, przeciw - 1, wstrzymało się 3. W 18. poprawce do art. 119 wnioskodawcy proponują nowe brzmienie ust. 9. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 19. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 20. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Janusz Cichoń, klub Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Panowie Premierzy! Ta poprawka dotyczy Prawa bankowego i reguluje kwestię wstrzymania transakcji bądź jej blokady w sytuacji, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, ale dotyczy to tylko Prawa bankowego. Dziwnym trafem podobnego zapisu nie ma, jeśli chodzi o SKOK-i.

Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 21. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę przyjął.

Pytanie zadaje pani poseł Genowefa Tokarska, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę tylko zauważyć, że projekt jest w ogóle bardzo obszerny, wymaga wielu zmian organizacyjnych, w tym również przystosowania systemów informatycznych. I bardzo, bardzo dużo instytucji, tzw. instytucji obowiązanych, zgłaszało to, wnioskowało kilkakrotnie o zmianę tego terminu, również na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. A pytanie jest proste: Dlaczego rządzący nie chcą wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom? Przecież wszystkim nam powinno zależeć na dobrym przygotowaniu tej ważnej ustawy, bo ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest naprawdę ważna. Mam dylemat, jak rozumieć słowo „rządzący” Rządzący, czyli Sejm - Sejm podejmuje decyzje, Sejm kontroluje Radę Ministrów. Ale pan minister Leszek Skiba odpowie pani poseł w imieniu rządzących. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Z tego powodu branża, instytucje finansowe, przedsiębiorcy generalnie są przygotowani do wdrożenia tej ustawy. Dziękuję bardzo. W takim razie możemy przystąpić do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Wysoka Izbo!

Czy wiecie państwo, ile miejsca zajmuje dyrektywa, która jest wdrażana za pomocą tej ustawy? Za każdym razem, implementując prawo unijne, implementujemy jakieś pomysły, które nie mają nic wspólnego z prawem unijnym. Produkujemy prawo tylko po to, aby było co czytać. Nie mówię, że ze zrozumieniem. Mamy jakiś problem i teraz może jest okazja, aby na to zwrócić uwagę. Zacznijmy tworzyć prawo, które ma sens. W czasie wystąpienia klubowego dawałem przykład jednego zapisu.

Dziękuję panu posłowi. W takim razie przystąpimy do głosowania. Dobrze. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2265, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2272-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Grzegorza Piechowiaka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym rozpatrzyła dwie poprawki, zgłoszone przez klub Platforma Obywatelska, i rekomenduje odrzucenie obu tych poprawek. Dziękuję panu posłowi. Przypominam, że chodzi o druk nr 2272. Nad poprawkami, które przedstawiła komisja, głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawki zostały zgłoszone do art. 3 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do Prawo o aktach stanu cywilnego. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Arkadiusz Marchewka, klub Platforma Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pod pretekstem umożliwienia zgłoszenia urodzin dziecka przez Internet tylnymi drzwiami wprowadzacie przepisy, które są kolejnym krokiem do inwigilowania Polaków i zaglądania w prywatne informacje o Polakach. Robicie to ekspresowo, bez żadnych konsultacji, nie wspominacie ani słowem w ocenie skutków regulacji dotyczącej tego projektu. Teraz do danych w rejestrze stanu cywilnego będą mogły sięgać nie tylko osoby, które są np. małżonkami, ale także służby nadzorowane przez PiS.

Przypomnę tylko zdanie na ten temat rzecznika praw obywatelskich, który powiedział tak: Forsowane rozwiązania uderzają w prawa jednostek i mogą być niezgodne z konstytucją, zwłaszcza z zasadą autonomii [[Dzwonek]] informacyjnej obywateli i prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przed całością zgłasza się poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Wysoka Izbo! Nie wiem, dlaczego państwo macie taką zasadę, że jeżeli uda wam się przygotować raz na jakiś czas jakąś w miarę rozsądną ustawę, to zawsze tak przekombinujecie, żeby opozycja nie mogła za nią głosować. Tak jest w tym przypadku. Całkiem rozsądna ustawa, która byłaby do przyjęcia bez problemu, ale coś was korciło, żeby jednak w niej pogmerać. Wprowadzacie możliwość, że służby będą mogły on-line ściągać wszystkie informacje z urzędów stanu cywilnego. Pytanie jest takie: Po co wam to, skoro były zasady, które jasno określały, że możecie to zrobić, ale w sposób, który jest pod jakąkolwiek kontrolą? Mało tego, jeszcze zrobiliście to w ten sposób, żeby zapis tak sugerował, że nawet przewodniczący komisji nie do końca wiedział, na czym to polega, że macie możliwość ściągania informacji on-line, a nie jednorazowo. Nie ma zgody na większe inwigilowanie społeczeństwa. Głos ma poseł Arkadiusz Marchewka, klub Platforma Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie ministrze, mam pytanie: Skoro to minister właściwy do spraw informatyzacji będzie wydawał służbom jednorazową zgodę na dostęp do danych o obywatelach, to proszę powiedzieć, panie ministrze, czy będzie to dotyczyło zgody na sprawdzanie danych każdego obywatela, czy będą to jednorazowe zgody na dostęp do wszystkiego, co tylko jest, czyli że ktoś np. w CBA będzie siedział przed komputerem i sprawdzał wszystkie dane, jakie są możliwe. Jeśli takie działania będą miały miejsce, to będzie to tylko i wyłącznie kolejny krok do tego, aby postępowało inwigilowanie społeczeństwa.

Wysoka Izbo!

Ta ustawa w żaden sposób tego nie dotyka ani nie zmienia. Dzięki temu, że jest to w drodze teletransmisji, pamiętajmy, że uzyskujemy też pełną rozliczalność tego, kto o jakie dane pyta w systemie rejestrów państwowych, który przechowuje akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa. Jest pełna rozliczalność, więc mamy pełną informację o tym, kto kiedy jakie dane przeglądał.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2272, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie to druk nr 2277-A. Proszę pana posła Jana Szewczaka o przedstawienie tego sprawozdania. Wysoka Izbo! Po licznych posiedzeniach podkomisji do spraw instytucji finansowych i posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych przyjmujemy dzisiaj dyrektywę unijną MiFID II, która wraz z załącznikami liczy ok. 1300 stron.

Przypominam, że chodzi o druk nr 2277.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Jakub Rutnicki, klub Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poprawka dotyczy alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W tym miejscu chciałem zapytać panią premier Beatę Szydło, czy tym alternatywnym funduszem inwestycyjnym są skandaliczne premie, które pani premier przyznała m.in. sobie - 65 tys. zł.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Chcę tylko odwołać się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Znowu wprowadzamy prawo unijne za pomocą innego dziwnego prawa. Kto z państwa przeczytał tę ustawę? Czy ktoś jeszcze? Pan przewodniczący też. Trzy osoby na tej sali przeczytały tę ustawę. Jestem przekonany, że pan minister też tego nie przeczytał.

Dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2277, wraz z jedną przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za głosowało 429, przeciw - 6, wstrzymał się 1 poseł. Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2315. Są pytania.

Wysoka Izbo! Ustawa o e-receptach to jest krok w dobrym kierunku. Informatyzacja w systemie ochrony zdrowia pozwoli uprościć bardzo skomplikowane procedury biurokratyczne. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia pan minister mówił o tym, że program pilotażowy, który w tej chwili dotyczy dwóch miast, Skierniewic i Siedlec, ma szansę być rozszerzony o kolejne miasta w innych regionach Polski. W związku z tym mam pytanie: Jakimi kryteriami będzie się kierowało ministerstwo, przyznając możliwość pilotażu w innych miastach? A inaczej to pytanie formułując: Co miasta muszą zrobić, aby dostać się do tego pilotażu? Dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2315, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 434, przeciw - 2, nikt się nie wstrzymał.

Wznawiam obrady. Wysoka Izbo! Przedstawię komunikat, informację po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego na dzień 1 marca br. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Jeżeli ktoś z państwa posłów jest zainteresowany, bardzo proszę.

Na tym zakończyliśmy oświadczenia.